Wznawiam posiedzenie. Proszę państwa, obecnie przystąpimy do stwierdzenia kworum. Posłowie zgłaszali, że przy pierwszym głosowaniu mają za mało czasu na zalogowanie się, więc poczekamy na to, żeby wszyscy posłowie mogli się zalogować. Proszę państwa, zwracam się do wszystkich posłów obecnych tutaj na sali, w innych salach i poza budynkiem Sejmu, o naciśnięcie dowolnego przycisku w celu sprawdzenia kworum.

Dziękuję i proszę o podanie wyników.

posiedzeniu bierze udział 458 posłów. Stwierdzam kworum. Z wnioskami formalnymi pan poseł Krzysztof Śmiszek. 1 minuta, panie pośle. Wysoka Izbo!

Oglądają nas miliony Polaków, w których narasta bunt. My, Lewica, będziemy patrzeć wam na ręce, na wasze partactwo, na waszą nieumiejętność pomocy Polakom. Dlatego uruchamiamy białą księgę, białą księgę niegodziwości i partactwa PiS-u.

Zajmijcie się wreszcie pracą.

Wczoraj na posiedzeniu Konwentu wyraźnie powiedziałam - i wszyscy państwo to wiedzieli, i z Prezydium, i z Konwentu - że czekaliśmy na opinie prawne, które dzisiaj spłynęły, część po południu.

Panie pośle, proszę więc nie mówić, że tymi projektami się nie zajmujemy, bo będziemy się zajmowali, ale. Wszystko więc dzieje się zgodnie z harmonogramem, o którym wszyscy państwo z Prezydium i z Konwentu wiedzieli.

Kto z pań i panów posłów jest za ogłoszeniem przerwy, proszę nacisnąć przycisk.

Sejm wniosek odrzucił. Wniosek formalny - pan poseł Borys Budka. Proszę bardzo, minuta. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! To, co dzisiaj dzieje się w parlamencie, tutaj, w Sejmie, to po raz kolejny prawdziwa wasza twarz. Przegraliście głosowanie, więc próbujecie na siłę wprowadzić kolejny projekt ustawy, ale tym samym pokazujecie, że dokładnie to samo zrobicie z wyborami, które przegracie. Właśnie temu ma służyć ten projekt ustawy, żeby zabezpieczyć was przed przegraną. Wnoszę o przerwę i przedstawienie Konwentowi Seniorów opinii prawnych o zgodności waszego projektu ustawy, który złożyliście kilka godzin temu, z konstytucją, czyli opinii Komisji Ustawodawczej, i z prawem europejskim, czyli opinii Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Zacznijcie wreszcie traktować Polaków poważnie. Kolejny dzień tracimy na wasze rozgrywki. Naprawdę, żyjecie w innym świecie. Tak zapatrzyliście się w tej nienawiści, w tej chęci władzy (Dzwonek), że zapomnieliście, czym żyją Polacy. Mamy na uwadze opinię Biura Analiz Sejmowych i taka opinia jest, panie pośle.

Proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Wnoszę zatem o odroczenie tych obrad, tego posiedzenia do chwili, kiedy państwo ogarniecie się i przedstawicie nam np. tę opinię, która, jak rozumiem, jest w posiadaniu pani marszałek, ale do tej pory pozostaje nieujawniona.

Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za odroczeniem posiedzenia, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił. Grupa posłów przedłożyła projekt ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., druk nr 328. Na posiedzeniu Konwentu Seniorów zgłoszono sprzeciw wobec propozycji uzupełnienia porządku dziennego o pierwsze czytanie tego projektu. Jest to, w myśl art. 173 ust. 4 regulaminu Sejmu, punkt sporny porządku dziennego. Propozycję uzupełnienia porządku dziennego o ten punkt poddam pod głosowanie. Przypominam, że zgodnie z art. 173 ust. 4 regulaminu Sejmu głosowanie to nie jest poprzedzone debatą ani zadawaniem pytań. Przyjęcie propozycji uzupełnienia porządku dziennego oznaczać będzie, że Sejm wyraził zgodę na skrócenie terminu, o którym mowa w art. 37 ust. 4 regulaminu Sejmu. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za uzupełnieniem porządku dziennego o punkt w brzmieniu: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., druk nr 328, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Sejm wniosek przyjął. Proponuję, aby Sejm wysłuchał w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 7. porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. (druk nr 328) Proszę pana posła Krzysztofa Sobolewskiego o przedstawienie uzasadnienia projektu ustawy. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Premierze! W imieniu wnioskodawców chciałbym przedstawić projekt ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., druk sejmowy nr 328. Wysoka Izbo! Nadrzędnym obowiązkiem państwa jest umożliwienie wszystkim uprawnionym obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej udziału w wyborach powszechnych na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. Uwzględniając panujące warunki światowej pandemii oraz ograniczenia w przemieszczaniu się, konieczne jest stworzenie ku temu odpowiedniego mechanizmu. Takim mechanizmem jest upowszechnienie trybu głosowania korespondencyjnego, co też zakłada projekt przedmiotowej ustawy.

Projekt nie ujmuje żadnych praw wyborczych, nie nakłada dodatkowych reżimów, a jedynie uprzystępnia obywatelom bezpieczne skorzystanie z konstytucyjnego czynnego prawa wyborczego. Przedstawiony projekt wychodzi naprzeciw potrzebom zorganizowania wyborów w konstytucyjnym terminie, z uwzględnieniem aktualnej sytuacji w kraju związanej z epidemią. Jest to niezbędna reakcja władzy ustawodawczej mająca na celu ochronę zdrowia i życia Polaków bez ograniczania czynnego prawa wyborczego. W proponowanym projekcie przyjęto, że każdy z uprawnionych do głosowania w celu oddania głosu otrzyma swój pakiet wyborczy i nie będzie zmuszony udawać się fizycznie do lokalu wyborczego. Nikt nie będzie musiał składać żadnych wniosków, zgłaszać potrzeby uzyskania pakietu wyborczego czy też podejmować jakiejkolwiek aktywności w celu uzyskania karty do głosowania. Państwo zapewni doręczenie dokumentów wyborczych.

Prawo pocztowe. Każdy wyborca potwierdzi swój głos stosownym oświadczeniem o dobrowolności i tajności głosowania.

Wyłoniony operator zapewni również odbiór pakietów ze skrzynek i ich transport do obwodowych komisji wyborczych celem przeliczenia głosów. Przeprowadzenie wyborów całościowo w formie trybu korespondencyjnego głosowania nie jest nowością, lecz jest czymś, co coraz częściej jest stosowane na świecie.

Nie stwierdzono poważniejszych uchybień, przy ponadmilionowym elektoracie frekwencja wyniosła ponad 50%. Wprowadzone tam zmiany dostosowujące regulacje prawne fundamentalne z punktu widzenia wzmacniania demokracji zostały przyjęte w ogólnym konsensusie i zrozumieniu nadzwyczajnych okoliczności faktycznych. Apele władz Bawarii o udział w głosowaniu korespondencyjnym spotkały się ze zrozumieniem wyborców. Przypomnę, iż całkiem niedawno parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej, dziś Koalicji Obywatelskiej, w sposób zdecydowany opowiadali się za taką formą wyborów. Panie pośle. Będzie czas dla pana i będzie pan mógł zabrać głos. W tej chwili ma głos wnioskodawca. gdzie w pracach nad wprowadzeniem całkowitego głosowania korespondencyjnego parlamentarzyści ci powoływali się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 20 lipca 2011 r., który ocenił, iż głosowanie korespondencyjne jest zgodne z konstytucją. 2 lata później powoływano się na te argumenty, podnosząc jednocześnie fakt, iż głosowanie korespondencyjne realizuje zasadę powszechności prawa wyborczego. Argumenty te w obliczu obecnej sytuacji są jeszcze bardziej aktualne, a przyjęcie podmiotowych uregulowań jest niezbędne w celu realizacji jednej z naczelnych zasad prawa wyborczego, tj. zasady powszechności. Wybory korespondencyjne? Oczywiście, że tak. Głosowanie korespondencyjne zagwarantuje wszystkim Polakom (Dzwonek), że będą mogli uczestniczyć w wyborach. Czyje to są słowa?

Zmiana ta jest również w pełni zgodna z obowiązującym prawem Unii Europejskiej oraz opiniami Rady Europy.

Poczta Polska jest instytucją o niekwestionowanym dorobku i tradycji.

Wskazał, że dla wyborcy tajność głosowań jest przywilejem, z którego może on skorzystać, choć nie ma takiego obowiązku. Oddanie głosu w sposób jawny, o ile nie stanowi formy agitacji wyborczej, nie wiąże się dla niego z żadnymi negatywnymi konsekwencjami prawnymi. Również dobrowolne poinformowanie o treści decyzji wyborczej innych osób, niezależnie od tego, czy ma miejsce przed wyborami, czy po wyborach, nie narusza zasady tajności głosowania. Tezę tę podtrzymał Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 18 lipca 2019 r., rozpatrując jeden z protestów wyborczych.

W tym miejscu chciałbym zaapelować do Wysokiej Izby o powściągnięcie emocji, zawieszenie rygorów walki politycznej, odłożenie na bok wszelkich uprzedzeń i partykularnych interesów partyjnych. W nadzwyczajnej sytuacji pokażmy, że potrafimy nie gorzej niż inne narody współdziałać dla dobra obywateli w pierwszej kolejności, a także w poszanowaniu fundamentalnych zasad demokracji. To nie czas na przepychanki, dezinformację i jałowe spory. Wszystkie siły polityczne winny teraz skupić się na polityce informacyjnej, docieraniu do obywateli z rzetelną informacją, uświadamianiu ich w zakresie przysługujących im praw wyborczych. Jak najszerszy udział w wyborach, jak najwyższa frekwencja wyborcza osiągnięta bez narażania zdrowia i życia obywateli winny być wspólnym celem całej klasy politycznej. Zaistniała sytuacja związana z epidemią koronawirusa wymusza na wszystkich wiele niedogodności i ograniczeń. Polacy mogą stanowić wzór dyscypliny dla innych narodów zmagających się z tą straszną zarazą. To wyjątkowa kampania - w cieniu spraw dalece ważniejszych, jednakże z równymi ograniczeniami dla wszystkich kandydatów. Zapewne każdy z nich chciałby prowadzić kampanię inaczej, aktywniej, ale jako politycy musimy dać przykład samodyscypliny i dostosowania do niedających się przewidzieć nadzwyczajnych warunków. Z uwagi na szczególną sytuację wywołaną rozprzestrzeniającym się koronawirusem oraz ważny interes państwa niezbędne jest natychmiastowe wejście w życie przedmiotowej ustawy. Warto przy tym dodać, iż Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 2006 r. uznał, że wprowadzanie zmian, nawet istotnych, w sytuacjach nadzwyczajnych jest możliwe w czasie ciszy legislacyjnej. Trudno wyobrazić sobie sytuację bardziej nadzwyczajną, niespodziewaną, a przy tym obiektywną i nakładającą na wszystkich, zarówno na administrację publiczną, jak i obywateli, ograniczenia, potrzebę dostosowania do zaistniałych okoliczności niźli tę, którą mamy aktualnie. Wysoka Izbo! Dziękuję, panie pośle. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła.

Proszę państwa, jesteśmy w trakcie dyskusji, więc bardzo państwa proszę, dokończmy to.

Pan poseł Łukasz Schreiber, bardzo proszę, w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Pani marszałek nie jest marszałkiem PiS-u, tylko marszałkiem Sejmu, pani marszałek. W odniesieniu do projektu ustawy może zostać przeprowadzone wysłuchanie publiczne. Uchwała w sprawie przeprowadzenia wysłuchania publicznego podejmowana jest przez komisję, do której projekt został skierowany do rozpatrzenia. Ale tu czas biegnie. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Panie Premierze! Wysoka Izbo!

Ale jesteśmy w czasie niezwykłym. W czasach takiego ciężkiego kryzysu nie można prowadzić tylko polityki ciepłej wody w kranie. Nie można podejmować tylko decyzji łatwych i popularnych. W takich czasach trzeba przede wszystkim podejmować decyzje odpowiedzialne, a kierować się tylko jednym: racją stanu. Wysoka Izbo! Chciałbym, zamiast omawiać ten projekt - to zrobił poseł wnioskodawca - odnieść się do kilku, nie powiem: kłamstw, powiem lżej: fake newsów, które wokół niego narosły. Otóż, Wysoka Izbo, chcę zapewnić, że rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego i większość parlamentarna pod przewodnictwem pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego mają dziś przede wszystkim na celu walczyć o zdrowie i życie Polaków, mają na celu walczyć o miejsca pracy i walczyć, by nie upadły polskie firmy. To jest nasze główne zadanie, temu też ten projekt zresztą służy, bo głosowanie korespondencyjne zamiast w lokalu wyborczym to jest właśnie także ochrona zdrowia Polaków. Podobno nie chcemy żadnego kompromisu. Wysoka Izbo, przecież kompromis leżał na stole: to propozycja, która być może miała swoje wady, ale miała też niezaprzeczalną zaletę - stabilizacji sytuacji, propozycja pana premiera Jarosława Gowina. Ona została odrzucona. Nikt nie robi teraz wyborów, a głosowanie korespondencyjne to szaleństwo. Wybory odbędą się w połowie kwietnia w Korei Południowej - kraju, który tak mocno został dotknięty przez pandemię koronawirusa, i to w lokalach wyborczych. Wybory można przesunąć. Wysoka Izbo!

A dlaczego? Wysoka Izbo, dlatego, aby nikt tym terminem konstytucyjnym, który został podany. Owszem, marszałek Sejmu ma prawo w pewnych granicach go przesunąć, ale tylko tyle. Stan nadzwyczajny jako remedium na wszystkie problemy.

To wprowadzenie stanu nadzwyczajnego niesie za sobą to, że nie można w tym czasie odbyć wyborów, i tylko tyle. Ja rozumiem, że jest to dla części wygodne, żeby miał on miejsce, że co 30 dni mielibyśmy się tu spotykać tylko po to, by toczyć awanturę o to, czy o kolejny miesiąc przesunąć wybory czy nie. A w ciągu tych 30 dni państwo będziecie zwolnieni z wszelkiej pracy, z domu jedynie udzielać wywiadów, nie brać za nic odpowiedzialności. To nie jest postawa odważnych ludzi. Szósty fake news, rzekoma kalkulacja wyborcza naszego obozu politycznego. Można powiedzieć krótko: Zawsze łatwo można poznać głupca. To ten, kto twierdzi, że wie, jak się skończą wybory. Otóż my tego nie wiemy. Chcemy, by te wybory się odbyły z jednego tylko powodu, i tylko jedna kalkulacja nam przyświeca. To chęć stabilizacji sytuacji w państwie, to chęć tego, byśmy wszyscy po tych wyborach, niezależnie od ich wyniku, razem z prezydentem nowo wybranym mogli zająć się tylko jednym i skupić się i zjednoczyć tylko dla jednej sprawy: walki z pandemią koronawirusa. Wysoka Izbo! Zwracam się z prośbą i apelem, byśmy do kryzysu (Dzwonek), który jest wywołany przez pandemię koronawirusa i który uderza w ochronę zdrowia oraz w zdrowie i życie Polaków, który uderza w gospodarkę, nie dodawali trzeciego kryzysu: kryzysu konstytucyjnego. Wnoszę i proszę Wysoką Izbę o poparcie tego projektu ustawy i składam wniosek w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość o natychmiastowe przejście do drugiego czytania. Dziękuję, panie pośle. Głos ma pan poseł Borys Budka, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Niestety po raz kolejny bawicie się w wielkie oszustwo. Od wielu dni oszukujecie Polaków, twierdząc, że będziecie im pomagać, a tymczasem dzień w dzień zajmujecie się waszymi wojenkami. Zajmujecie się tym, na czym naprawdę wam zależy, czyli utrzymaniem władzy za wszelką cenę. Przecież to kuriozalne, że przedstawiciel komitetu wyborczego prezydenta Andrzeja Dudy jest teraz przedstawicielem wnioskodawców. Oszukiwaliście, oszukujecie i będziecie oszukiwać. Przegraliście dzisiaj głosowanie, to złamaliście kręgosłupy, być może szantażem, być może kupnem, po to, by jeszcze raz przedłożyć taki projekt ustawy. Zemści się to, że nie chcecie rozmawiać o istotnych problemach Polek i Polaków. Zemści się to, że oszukujecie, twierdząc z jednej strony, że wybory nie mogą się odbyć, ale z drugiej strony na siłę dążąc do rozprzestrzenienia się tego wirusa. Jest pan minister Szumowski, który tak wiele mówi o klauzuli sumienia, o przysiędze Hipokratesa. I przed chwilą głosowaliście za tym, żeby rozprzestrzeniać dalej wirusa. Głosowaliście za tym, by wbrew logice, wbrew zdrowemu rozsądkowi, ale przede wszystkim elementarnej etyce wysyłać ludzi czasami nawet na śmierć, bo nie macie żadnego szacunku.

Jest mi po ludzku wstyd. Jest mi po ludzku wstyd, że przyszło nam zasiadać w parlamencie z takimi ludźmi, ludźmi, którzy są nieczuli na błagania tych, którzy dzisiaj wołają o pomoc: matek, ojców, przedsiębiorców, pracowników. Kolejny dzień tracicie na to, by utrzymać się przy władzy. To jest żenujący spektakl. To jest żenujący spektakl pokazujący, jak ta władza gnije od środka, jak łamiecie sobie nawzajem kręgosłupy. Niektórzy wasi koledzy jeszcze niedawno mówili: dziesiątego nie da się zrobić wyborów. Zrobicie je siedemnastego? To jest początek waszego końca. Polacy wam tego nie zapomną. Ale przede wszystkim nie zapomną wam tego ci, których zdrowie i życie narażacie. Nie zapomną wam tego pracownicy Poczty Polskiej. Nie zapomną wam tego ci, którzy będą musieli zajmować się liczeniem głosów. To jedno wielkie oszustwo. Wasza narracja oparta jest na oszustwie. Oszukujecie rano, w południe i wieczorem. Oszukujecie, bo władza jest dla was najważniejsza. Dzisiaj staliście się elementem zupełnie obcym dla społeczeństwa, bo wy nie widzicie realnych potrzeb Polaków, nie widzicie nawet tego, że blisko 90% ludzi boi się głosować. Wy każdego dnia za te 2 mld zł, które mogły być przeznaczone na służbę zdrowia, siejecie propagandę i kłamstwo. Będziecie teraz udawać, jak to troszczycie się o zdrowie Polaków. A nie lepiej te środki przeznaczyć chociażby na ochronę służby zdrowia? Za grosz nie macie wstydu. Ta władza się skończy prędzej czy później, ale tacy ludzie jak wy przejdą do historii. Przejdą do tej niechlubnej historii, gdzie łamiąc sumienia tym, którzy jeszcze je być może kiedyś mieli, w imię własnego interesu poświęcacie zdrowie i życie Polaków. Jesteście tak chorzy na władzę, że nie widzicie rzeczy oczywistych. Zgodnie z polską konstytucją można przesunąć termin wyborów, wprowadzając stan klęski nadzwyczajnej, ale wy tego nie zrobicie, bo wiecie, że przegracie. Wy tego nie zrobicie również dlatego, że nie chcecie płacić odszkodowań. Nagle okazuje się, że budżet jest pusty, król jest nagi. I powiem wam szczerze, że jak obserwuję te ostatnie dni, to jest mi tak po ludzku przykro. Przykro, że dożyłem czasów, w których większość parlamentarną stanowią obłudni cynicy, ludzie, którzy często powołując się na Boga, na interes narodu, na rację stanu, kreują się na świętych, a są zepsuci do kości. Dziękuję, panie pośle.

Pan poseł Krzysztof Śmiszek, klub parlamentarny Lewica. Wysoka Izbo! Zanim przejdę do prezentacji stanowiska Lewicy, chciałbym przede wszystkim powiedzieć naszym rodakom, którzy oglądają nas teraz poprzez środki masowego przekazu, że dzisiaj mamy dzień świstaka. Kilka godzin temu Sejm powiedział „nie” debacie o wyborach. A co mamy teraz? Debatę o wyborach. Dzisiaj Sejm został zagoniony przez PiS-owską większość do bezsensownej rozmowy o głosowaniu korespondencyjnym, nie o wsparciu dla was. Zmarnowaliśmy kolejny dzień. Marnujemy bezcenny czas. Ten Sejm od tygodnia nie przyjął żadnego porządnego rozwiązania, które wychodziłoby naprzeciw waszym problemom. Za to przerabiamy już kolejną wersję ustawy o wyborach. Ten sam Sejm kilka dni temu pozbawił Polki i Polaków wsparcia, które wypracował dla nich Senat. Tak, chcę, żeby Polki i Polacy usłyszeli, że PiS, odrzucając poprawki Senatu, wyrzucił do kosza pomoc dla pracowników i przedsiębiorców. Zamiast tego zgodziliście się na wydanie miliardów na system bankowy oraz pokrycie ubezpieczeń dla księży. Widać, jakie ta władza ma priorytety. Widać, kto jest dla was bohaterem. Dzisiaj zamiast o konkretach będziemy rozmawiać o wyborach. Czy wy nie rozumiecie, że nikogo te wybory nie obchodzą? Nikogo. Czy wy nie rozumiecie, że kartą do głosowania nie da się najeść, że karta do głosowania nie opłaci rachunków za gaz czy prąd? Wasz projekt ustawy łamie wszelkie reguły przyzwoitości. To, że dziś procedujemy nad tą ustawą, jest splunięciem w twarz naszym rodakom. PiS działa w myśl zasady: Nie mają chleba? W czasie, kiedy dziesiątki innych krajów odwołują wybory, bawicie się publicznymi pieniędzmi. Ile będą kosztowały te wybory? Kolejny projekt ustawy, który przedstawiacie, to kpina. Kpina z konstytucji, kpina z logiki, kpina z obywateli i kpina z rozumu. Za kilka dni rocznica katastrofy smoleńskiej. Wszyscy pamiętamy ostatnie słowa z kokpitu: dasz radę, zmieścisz się. Dacie radę, zagłosujcie. A potem? Najważniejsze, że Andrzej Duda zostanie prezydentem. Proszę mi wytłumaczyć, jak wy chcecie zorganizować te wybory, tak aby pracownicy poczty byli bezpieczni. Każdy listonosz będzie mieć kontakt z ponad 1 tys. osób, a to tylko w odniesieniu do dostarczenia pakietów wyborczych, oprócz codziennych innych obowiązków. A może chcecie zaangażować do wyborów wojsko? Powiedzmy sobie to wprost. Powinien być procedowany w trybie przewidzianym dla kodeksów, z komisją nadzwyczajną, z ekspertami i odpowiednimi terminami. Co najważniejsze, ten projekt ustawy zmienia konstytucję. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że apelowanie do rządu o szacunek wobec prawa czy konstytucji nie ma żadnego sensu. Dlatego zwracam się do waszego poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo obywateli. Igracie z życiem i zdrowiem Polaków. Przedstawiony projekt przepisów wyborczych to ani przepisy, ani wyborcze. To regulamin prymitywnej ruletki, gdzie stawką są demokracja, życie i zdrowie Polaków.

Proponuję nie bawić się w tej Izbie w udawanie pracy, ale przyjąć w projekcie, że wszyscy nasze karty do głosowania pobieramy na Nowogrodzkiej, a w szczególności, że tam je wysyłamy. Tam już będą wiedzieć, co z tymi kartami zrobić. Albo jeszcze lepiej: zagłosujmy w tych wyborach drogą SMS-ową. Można? Można. Przecież w państwie PiS można głosować w każdy sposób. Ważne, żeby wepchnąć Andrzeja Dudę ponownie na prezydencki stołek. Tymi wyborami będzie rządzić zasada: kto ma kluczyk do skrzynki, ten ma władzę. I w zasadzie na tym można by skończyć, gdyby nie to, że kwestia wyborów nikogo nie obchodzi. Ja wam coś powiem. Chcecie, żeby Poczta Polska dostarczyła 30 mln kart do głosowania? Jak na razie Poczta Polska dostarcza każdego dnia miliony innych listów: wypowiedzeń z pracy i wezwań do zapłaty, bo tak właśnie wygląda dzisiaj rzeczywistość poza salą sejmową. Zamiast liczyć głosy, policzcie już dzisiaj tych ludzi, którzy potrzebują pomocy. Rząd powinien pracować dniami i nocami. I faktycznie na Nowogrodzkiej od kilku dni trwają nocne narady najważniejszych polityków PiS-u i rządu, ale oni nie myślą i nie debatują o tym, jak pomóc Polkom i Polakom. Oni dzisiaj przeciągają linę między prezesem Kaczyńskim a premierem Gowinem. Na zakończenie chciałbym powiedzieć jeszcze jedno: to wy rządzicie, to wy decydujecie o tym, czym danego dnia ma zajmować się ta Izba. I właśnie dlatego każdy zwolniony z pracy, każda zamknięta firma, każdy niepotrzebny przypadek zakażenia i każda śmierć, której można było uniknąć, obciąża wasze sumienie.

Wysoka Izbo! Ta ustawa to utrwalacz władzy, władzy, która oderwała się od obywatela, władzy, która oderwała się od rzeczywistości, która zapomniała, do czego jest powołana. Składaliście przysięgę: służyć narodowi, dbać o dobro i pomyślność obywateli, a ta ustawa jest po to, żeby wykorzystać obywatela dla utrwalenia swojej władzy. To jest prostsze rozwiązanie: napisać jeden artykuł, że Andrzej Duda jest dożywotnio prezydentem Polski. Przynajmniej nie będziecie narażać całej Polski, wszystkich obywateli Rzeczypospolitej na niebezpieczeństwo. Robicie te wybory, bo boicie się, że na jesień czy może na wiosnę przyszłego roku nie będziecie mieć poparcia i nie wygracie już wyborów. Robicie te wybory dlatego, że straciliście słuch społeczny. Nie interesują was sprawy najważniejsze, te, które dzisiaj martwią tysiące, miliony polskich rodzin: Jak przeżyć? Jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny? Jak się nie zarazić? Jak otrzymać pomoc? Jak mają wytrzymać pielęgniarki, lekarze i ratownicy, którzy są w szpitalach? Jak uratować miejsce pracy? Jak uratować swoją firmę? To są najczęściej zadawane pytania. Wy ich kompletnie nie widzicie.

Władza jest po to, żeby rozwiązywać problemy obywateli, a nie je mnożyć. Władza jest po to, żeby dbać o bezpieczeństwo, a nie narażać życia i zdrowia. Władza jest po to, żeby być odpowiedzialnym i roztropnym, a tu nie ma roztropności, nie ma przyzwoitości i nie ma odpowiedzialności - za grosz. Utraciliście te wszystkie przymioty, te wszystkie wartości. Boicie się utraty władzy i nie wyobrażacie sobie tej sytuacji, ale tylko dlatego, że jesteście do niej przyspawani, że to jest dla was cel sam w sobie. Nie zważacie na opinie ekspertów, naukowców, np. Komitet Bioetyki przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk mówi wyraźnie, że przeprowadzenie tych wyborów w zarządzonym terminie jest moralnie nieodpowiedzialne i prawnie niedopuszczalne, przeprowadzenie i przygotowanie tych wyborów będzie naruszało konstytucyjnie chronione prawa człowieka i obywatela: prawo do życia i zdrowia oraz prawa wyborcze. Nie zważacie na list Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, którzy mówią: i sposób bezpośredni głosowania, i sposób korespondencyjny zagrażają dobrostanowi obywateli, zagrażają zdrowiu, bo zdrowie to dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny.

Nie będą to wybory równe, nie będą to wybory bezpośrednie i nie będą przeprowadzone w głosowaniu tajnym, czyli wszystkie przymioty, które powinny mieć wybory, w których wybiera się prezydenta Rzeczypospolitej, będą naruszone. Utraciliście ten instynkt, który kiedyś was doprowadził do władzy, ale przyzwyczailiście się, że ta władza jest dla was świętością. To chcę wam jeszcze raz powtórzyć: święte są życie i zdrowie, święte są życie i zdrowie obywateli Rzeczypospolitej, a nie data 10 maja, 17 maja czy jakikolwiek inny termin w maju, który naraża to życie i zdrowie na szwank, na utratę, na śmierć. Zapomnieliście o tym, bo straciliście to, co było dla was kiedyś wartością. Na koniec chcę się odwołać do posłów PiS-u, nie powołując się na wyroki Trybunału Konstytucyjnego, orzeczenia Sądu Najwyższego, ale powołując się, apelując do najwyższego trybunału, do waszego sumienia, nie jako lekarz, kandydat na prezydenta, poseł czy polityk, ale jako jeden z obywateli Rzeczypospolitej. Czy macie tę odwagę, która na oślep będzie pędzić, patologiczną, która narazi życie i zdrowie naszych rodaków, która narazi życie i zdrowie (Dzwonek) na szwank? Dziękuję, panie pośle.

Zgodnie z art. 184 ust. 3b wniosek formalny nie może być zgłoszony, jeżeli wniosek z nim tożsamy został już odrzucony przez Sejm. Przypominam panu, że taki wniosek został złożony i został odrzucony przez Sejm.

Bardzo proszę, pan poseł Krzysztof Bosak. Pani Marszałek! Chciałem powiedzieć: panie premierze, panie prezesie, ale wszyscy wyszli. Pani Marszałek! Szanowni Posłowie, którzy przebywają na sali i słuchają nas przez internetowy system obrad! Drodzy Obywatele! Polacy dzisiaj nie czekają na dyskusję o detalach Kodeksu wyborczego. Polacy dzisiaj czekają na rozwiązania poprawiające jakość ochrony zdrowia, na wsparcie dla pracowników, na wsparcie dla przedsiębiorców, realne, a nie na papierową, biurokratyczną tarczę antykryzysową. Tymczasem partia rządząca, która ma większość w Izbie, wciąga nas w dyskusję o sposobie przeprowadzenia wyborów, w dyskusję, co do której partia ma świadomość, że Polacy jej nie oczekują. Jeżeli tę dyskusję musimy prowadzić, to dobrze, odniesiemy się także do tego, co tutaj państwo proponujecie. A więc po kolei 10 rzeczy, które są nieprawdą w tym, co proponujecie, i w tym, o czym mówicie. Po pierwsze, nie zmienia się reguł w trakcie gry. To, co robicie, jest nieuczciwe, to, co robicie, jest nie fair. Po drugie, nie jest prawdą, że nie da się przesunąć wyborów. Literalnie tu przed chwilą przede mną poseł i minister w kancelarii premiera Schreiber wprowadzał Polaków w błąd, wymachując konstytucją. W konstytucji są oczywiste przepisy, których wystarczy użyć, żeby przesunąć wybory.

Oczywiście. Ale przesunąć wybory, wprowadzić stan nadzwyczajny po to, żeby chronić zdrowie i życie obywateli? Konstytucja daje taką możliwość, w związku z czym nie manipulujcie państwo. Trzecia sprawa. Złożyliście drugi raz projekt w tej samej sprawie, który przerobiliście. Piszecie prawo na kolanie, panie pośle. Sam fakt, że przegraliście głosowanie w Sejmie, dał wam dodatkowe godziny, kiedy wasi prawnicy na kolanie poprawiali ten projekt, dopisywali do niego nowe rzeczy, których wcześniej nie było. Czwarta sprawa. Nie jest prawdą, że sami w to wierzycie. Nie jest prawdą, że sami w to wierzycie, bo rozmawiamy z wami w kuluarach i wiemy, że wielu waszych posłów bardzo boi się terminu 10 maja. Macie wbrew pozorom w swoich ławach bardzo wielu rozsądnych posłów, którzy wiedzą, że to zły pomysł, żeby robić wtedy wybory. Następna sprawa. Wiecie o tym.

Kolejna sprawa. Nie jest tak, żeby poczta była na to przygotowana, choć chcecie sprawiać takie wrażenie. Gdybyście byli przygotowani na to i gdybyście byli przekonani, że poczta jest przygotowana, żeby ten proces obsłużyć, to nie zmienilibyście właśnie szefa Poczty Polskiej, zastępując go wiceministrem obrony narodowej, zresztą zaufanym człowiekiem ministra Błaszczaka. Siódma sprawa, o której chcę powiedzieć. To, co proponujecie, odbierze prawa polityczne Polakom. Dużo mówicie o niemożliwości wprowadzenia stanu nadzwyczajnego. Ministrowie pana prezydenta Andrzeja Dudy dezinformują Polaków, mówiąc, że przesłanki konstytucyjne nie są spełnione. Jest to nieprawdą, bo wystarczy, że środki konstytucyjne nie są wystarczające, że jest zagrożenie, i wówczas można podjąć polityczną decyzję o wprowadzeniu stanu nadzwyczajnego. Natomiast mało mówicie lub w ogóle nie mówicie o tym, czemu służy instytucja stanu nadzwyczajnego w konstytucji. Brak wyborów w stanie nadzwyczajnym służy ochronie praw politycznych Polaków: do głosowania, do prowadzenia kampanii wyborczej. Może Polacy nie czekają, żebyśmy prowadzili kampanię wyborczą, ale to są jednak nasze prawa polityczne. Przeprowadzając wybory 10 maja, wszystkim moim zwolennikom i zwolennikom innych kontrkandydatów z opozycji odbieracie możliwość prowadzenia normalnej kampanii wyborczej. Zostało mi 30 sekund, więc będę mówił szybko. Obniżycie legitymację prezydenta, ktokolwiek zostanie wybrany. Jeśli wam się uda i wybrany zostanie prezydent Andrzej Duda, jego mandat będzie podważany. Dziewiąta sprawa. Projektodawcą, osobą referującą projekt jest pan, panie pośle, pełnomocnik komitetu wyborczego Andrzeja Dudy. Czy można sobie wyobrazić większy konflikt interesów niż to, że projekt zmiany prawa wyborczego proponuje pełnomocnik jednego z kandydatów? Ostatnia sprawa. 5 sekund mi zostało.

Informuję panie i panów posłów, iż Prezydium Sejmu na podstawie art. 39 ust. 1 regulaminu Sejmu ustaliło w tym punkcie limit 10 pytań dla klubów według następującego parytetu: Prawo i Sprawiedliwość - pięć, Koalicja Obywatelska - trzy, Lewica - jedno, PSL - jedno. Lista posłów zgłoszonych do pytań - jeszcze jej nie mamy. Zgłosili się następujący posłowie. Zamykam listę zgłoszeń. Jako pierwszy pan poseł Marcin Kierwiński, klub Koalicji Obywatelskiej. Wysoka Izbo! Kilka godzin temu pan premier Morawiecki tutaj, w tej Izbie, powiedział, że spodziewamy się, że szczyt zachorowań jest przed nami, będzie w maju lub w czerwcu. Pytam kolegów z PiS-u. Ano chcecie zrobić wybory. Chcecie Polakom zorganizować wybory. Ale tak naprawdę tym kodeksem chcecie Polakom ukraść wybory, ukraść wolne, niezależne wybory. Ten system, który wprowadzacie, ten Kodeks wyborczy - patrzę tu na pana posła sprawozdawcę - to nic innego jak kodeks, który umożliwia masowe fałszowanie wyborów. Zamiast pomocy dla firm, zamiast pomocy dla pracowników, zamiast pomocy dla służby zdrowia wy chcecie pomóc tylko i wyłącznie sobie. Chcecie zorganizować te wybory za wszelką cenę, nawet po trupach. Wtedy, kiedy to będzie wam potrzebne, chcecie ustawić ich wynik.

Wysoka Izbo! PiS marnuje dzisiejszy dzień na targi polityczne - w momencie, kiedy miliony Polek i Polaków przeżyło ten dzień w obawie o swoje zdrowie, o swoje życie, o swoją pracę, o to, co stanie się z ich firmą. Nie wiedzą także, czy ich dzieci podejdą do matury. Nie interesują was ludzkie dramaty. Interesuje was tylko to, czy dalej będziecie rządzić, czy będziecie mieć prezydenta - za wszelką cenę, być może za cenę zdrowia i życia Polaków. Próbujecie wmówić nam, że wybory mogą zostać przeprowadzone w sposób uczciwy, demokratyczny. To może mi ktoś wyjaśni, w jaki cudowny sposób pod projektem ustawy podpisała się własnoręcznie posłanka, która głosowała zdalnie ze swojego okręgu. Powiedzcie mi, w jaki sposób to się stało. Czy wojsko będzie nam organizowało wybory?

Panie Marszałku! Ale przede wszystkim wy, Polacy, ponieważ to jest szalenie istotny dzień dzisiaj, to jest naprawdę kluczowy dzień dla naszej demokracji. Bo z głosowaniem korespondencyjnym jest jak z nożem: może służyć do krojenia chleba, ale może też służyć do zabijania. I dzisiaj posłowie, którzy będą głosować za tą ustawą, chcą zabić polską demokrację. Chcecie przeprowadzić zamach stanu, bo to głosowanie będzie jednym wielkim oszustwem. Dobrze wiecie, że ono jest technicznie nie do zrobienia.

Polacy tego nie chcą. Chcecie te pakiety wrzucać do skrzynek domowych, których nikt nie będzie kontrolował. Wybory będzie robił rząd dla siebie. Wyrzucacie Kodeks wyborczy, dajecie specustawę, wyrzucacie Państwową Komisję Wyborczą, a wprowadzacie rządową komisję. Proszę, pan poseł Piotr Zgorzelski, PSL-Kukiz15. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Polska tym samym staje się państwem stanu wyjątkowego bez stanu wyjątkowego. Naruszyliście zasadę nieprzeprowadzania istotnych zmian w Kodeksie wyborczym na 6 miesięcy przed wyborami. To jest zmiana prawa wyborczego w trakcie trwania procesu wyborczego, to wszystko po prostu musi się źle skończyć. Na koniec, parafrazując Winstona Churchilla, chcę wam powiedzieć: Mieliście do wyboru przełożenie terminu lub hańbę.

Pani marszałek, to, że siedzi pani tyłem do orła, nie znaczy, że może pani go lekceważyć. Dzisiaj łamiecie konstytucję, łamiecie polskie ustawy i polskie prawo. Chciałbym natomiast zwrócić uwagę na coś szczególnie istotnego, coś, o czym wszyscy musimy pamiętać. Dzisiaj 37 posłów PiS-u podpisało się pod tym haniebnym projektem. Jak to możliwe, skoro ci posłowie informują, że są w swoich okręgach wyborczych? Jak to możliwe, że np. pani Violetta Porowska albo pani Barbara Dziuk, albo pan poseł Robert Telus, którzy informują, że są dzisiaj w swoich okręgach wyborczych i głosują zdalnie, podpisali projekt ustawy, który złożyliście w Sejmie? To jest jawne fałszerstwo.

Dziękuję, panie pośle.

Rząd próbuje na siłę przeprowadzić wybory prezydenckie, dlatego że zdaje sobie sprawę, że to jest ostatni moment, żeby Prawo i Sprawiedliwość miało szansę wygrać jakiekolwiek wybory, i to nie z powodu przedsiębiorców, którzy za chwilę będą masowo bankrutować, ale z powodu Polaków, którzy za chwilę będą masowo bankrutować razem z przedsiębiorcami, tracąc swoje miejsca pracy. Tymczasem w odpowiedzi premier Morawiecki dzisiaj zaproponował trzy nowe podatki Unii Europejskiej, zaproponował likwidację rajów podatkowych na całym świecie. Czy wy nie rozumiecie, że jak tak dalej pójdzie, to nie będzie z kogo ściągać tych podatków?

Do głosowania nad tymi wnioskami przystąpimy niezwłocznie. Odrzucenie tego wniosku będzie oznaczać, że Sejm podjął decyzję o niezwłocznym przystąpieniu do drugiego czytania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu ustawy zawartego w druku nr 328, zechce nacisnąć przycisk.

Stwierdzam, że Sejm wniosek odrzucił, a tym samym podjął decyzję o niezwłocznym przystąpieniu do drugiego czytania projektu ustawy. Przystępujemy do drugiego czytania projektu ustawy. Proszę bardzo, wniosek formalny. Wysoka Izbo! Na podstawie art. 184 regulaminu Sejmu zgłaszam wniosek formalny o przerwę w posiedzeniu Sejmu w celu zwołania Konwentu Seniorów i dodania do porządku obrad punktu dotyczącego rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zobowiązania Rady Ministrów do wprowadzenia stanu klęski żywiołowej. Szanowni Państwo! Mamy dobrą konstytucję, wystarczy jej nie łamać. Jest w niej zapis o możliwości wprowadzenia stanu klęski żywiołowej. Ten zapis należy wykorzystać, dlatego że epidemia to także klęska żywiołowa. Najwyższy czas z tego zapisu skorzystać i zakończyć debatę na temat wyborów korespondencyjnych, zwykłych, telepatycznych, jakichkolwiek. Dziś musimy rozmawiać o tym, co ważne dla Polek i Polaków, o zasiłku kryzysowym, o podwyższeniu zasiłków dla bezrobotnych, o ratowaniu miejsc pracy, o objęciu wszystkich pracowników ochroną, o przełożeniu matur, przełożeniu egzaminów. Polki i Polacy czekają dzisiaj, aż my i wy z tego miejsca powiemy: trzymajcie się, damy radę. Pani poseł, dziękuję. Zgodnie z regulaminem tego wniosku nie poddaje się pod głosowanie i powinna pani o tym wiedzieć. Przystępujemy do drugiego czytania projektu ustawy. Pan poseł Krzysztof Śmiszek, klub parlamentarny Lewica.

Wysoka Izbo! Składam wniosek formalny o ogłoszenie przerwy i zwołanie Konwentu Seniorów. Otóż dzisiaj podczas debaty z udziałem pana premiera Morawieckiego chcieliśmy zdalnie zadać pytanie. Pani marszałek, pamiętam, obiecywała, że system będzie działał prawidłowo, że wszystko jest dobrze, natomiast kilku posłów nie mogło zagłosować. Mogliście państwo poczekać dobrych kilka minut, bo za chwilę, po debacie, mogliśmy zadać te pytania. Ale państwo nie czekali. Jest tak, że państwo nam odbieracie prawo do uczestniczenia w debacie. Mam prośbę, żeby pani chwilę posłuchała, pani marszałek, bo ten system informatyczny nie działa tak, jak działać powinien. Ja dzisiaj specjalnie przyjechałem z Łodzi, ponieważ ten system nie działa, a chciałem panu premierowi zadać konkretne pytania. A chciałbym zadać pytania dotyczące tego, dlaczego narażacie ludzi na śmierć i doprowadziliście do krytycznej sytuacji.

Dziękuję bardzo, panie pośle. Bardzo pana przepraszam. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Dzisiaj debatujemy nad projektem bardzo ważnym, projektem, który jest skrajnie niekonstytucyjny i skrajnie antypaństwowy, jednak debatujemy nad tym projektem nawet bez podstawowych opinii o tym, czy projekt jest zgodny z konstytucją. Debatujemy też bez opinii lekarzy, ludzi, którzy znają się na tym i wiedzą, czy takie głosowanie jest bezpieczne dla Polaków. Chciałbym przypomnieć, że 15 marca w Bawarii odbyły się wybory lokalne, na które często państwo się powołują. Do tego dnia w Niemczech zgłoszono 7046 przypadków zarażenia koronawirusem, z czego 1139 przypadało na Bawarię.

Panie pośle, to nie jest wniosek formalny. Informuję pana, że nadużywa pan tej mównicy. Poinformowałam państwa, że wnioski formalne o przerwę były kilkukrotnie zgłaszane i głosowane.

To nie są wnioski formalne.

Państwo nie słuchaliście.

Dziękuję, panie pośle. Jeżeli pan nie chce zabrać głosu, panie pośle.

To przepraszam, 5 minut. Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Panie pośle, bardzo proszę. Niestety wnioski formalne nie są przez panią nawet poddawane pod głosowanie. To, o czym mówi pan poseł Tomczyk, to oczywista oczywistość, jak powiedziałby klasyk. Ale tutaj chodzi tylko i wyłącznie o to, żebyście państwo kolanem jak najszybciej dopchnęli kolejny bubel prawny. Nawet nie odpowiadacie na żadne pytania, bo przyzwoitość to jest cecha wam obca. Uczciwość to jest cecha wam obca. Jakaś sportowa rywalizacja to jest cecha wam obca. Wy za wszelką cenę chcecie utrzymać tę władzę. Po trupach do celu - to będzie maksyma tych wyborów. To wstyd, że większość parlamentarna jest w stanie myśleć tylko o sobie. To wstyd, że państwo nie potraficie wsłuchać się w głos tych wszystkich, również waszych, wyborców, którzy nie chcą narażać swojego zdrowia i życia. To wstyd, że próbujecie doprowadzić do wielkiej kompromitacji polskiego systemu wyborczego. Poczta nie jest w stanie na czas doręczać przesyłek w tej chwili, bo nie ma listonoszy, a wy chcecie robić korespondencyjne wybory? Wy chcecie, żeby w gminie była jedna komisja wyborcza, a w Warszawie jedna komisja w dzielnicy? To będzie wstyd na całą Europę, na całą Polskę. Ale przede wszystkim dziwi mnie to milczenie prezydenta Andrzeja Dudy. Rozumiem, że jego pełnomocnik zabiera tutaj głos, bo pan prezydent tak kurczowo trzyma się władzy.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Ten projekt jest nieprzyzwoity. Ten projekt wprowadza zasady, które spowodują, że tych wyborów nie będzie nikt przyzwoity uznawał.

Zgodnie z polską konstytucją już dawno premier Morawiecki powinien wnioskować o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej. Ograniczacie prawa obywatelskie każdego dnia, zakazaliście nawet wstępu do lasu, ale chcecie ludzi wysłać tym razem do skrzynek pocztowych. Kolejki, które będą się tam tworzyć, będą dużo większym zagrożeniem aniżeli zwykłe spacery w lesie. Ale nie cofniecie się przed niczym, bo już zapomnieliście, że jesteście częścią opinii publicznej. Teraz jest już podział: wy i cała reszta. Przestaliście się liczyć z głosem opinii publicznej, bo przegrywacie. Nawet jeżeli jakimś cudem jeszcze wygracie te wybory, to jest to, panie prezesie, początek końca.

Proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Cytuję: Setki razy tłumaczyłem: w komisji, w mediach, tutaj na Twitterze czy na sali plenarnej: głosowanie korespondencyjne niesie ryzyko fałszerstw - patrz: powtórzone wybory w Austrii rok temu - i jest dozwolone jedynie w 13 na 28 krajów Unii Europejskiej podczas wyborów samorządowych. To ja pytam: Gdzie jest prawda?

Szanowni Państwo! Art. 128 ust. 2 konstytucji ma charakter jednorazowy, a to, co zawarliście państwo w przepisach projektu tej ustawy, że marszałek Sejmu może zmienić postanowienie o zarządzeniu daty wyborów, to jest kpina. To jest kpina z konstytucji, to jest kpina nawet z logiki i ze zdrowego rozsądku. Przepis art. 128 ust. 2 to kwestia jednorazowego wyznaczenia daty wyborów i wyczerpuje się po wydaniu pierwotnego postanowienia o takim zarządzeniu.

Czy ma to coś wspólnego z wyborami, które są wolne, powszechne, równe? A co z wyborami tajnymi?

Co się stanie, jeśli nie odbiorę karty ze swojej skrzynki pocztowej, a termin wyborów minie? Czy to znaczy, że ukradłem kartę wyborczą? Czy to znaczy, że ją zniszczyłem? Ewentualnie pewnie już wy będziecie wiedzieć dzięki pomocy listonoszy, że taką kartę dostałem, czyli grożą mi 3 lata pozbawienia wolności za nieodebranie karty wyborczej ze swojej skrzynki pocztowej. To, co jest zaprezentowane w tym projekcie, to jest kpina. Przecież ta ustawa składa się właściwie z samych delegacji do wydawania aktów wykonawczych przez kolejnych ministrów, przez ministra do spraw aktywów państwowych. Gdzie są projekty rozporządzeń, na mocy których będziemy organizować proces wyborczy? To jest kuriozum na skalę światową, że zamiast za pomocą przepisów ustawowych robimy wybory za pomocą przepisów rangi rozporządzenia. Jaka jest rola Państwowej Komisji Wyborczej? Ta rola jest sprowadzona do roli biernego obserwatora.

Dzisiaj, zamiast zajmować się kwestiami palącymi. Przecież każdy z nas dostaje dzisiaj na swoje skrzynki pocztowe maile, dzwonią ludzie do naszych biur poselskich, piszą maile, piszą SMS-y: zamykają mi firmę, straciłem pracę, mam umowę zlecenie, nie dostałem zasiłku, muszę opłacić rachunki, dzieci muszą dostać coś do jedzenia na kolację czy na śniadanie. Dzisiaj o tym musimy rozmawiać, a my dzisiaj rozmawiamy o jakichś fantasmagoriach wyborczych, my dzisiaj rozmawiamy o tym, jak minister Sasin będzie nam organizował wybory. Naprawdę powiedzcie szczerze, o co w tym wszystkim chodzi. Kto dzisiaj o zdrowym umyśle będzie chciał pójść na wybory, wyjmować te karty ze skrzynek, chodzić gdzieś, szukać po dzielnicach, po mieście, po gminie odpowiedniej skrzynki wyborczej, do której będziemy to wrzucać?

Otóż mamy tutaj naprawdę absurdalną sytuację.

Oczywiście to jest istotne, natomiast Polacy za chwilę mogą mieć problem ze zwykłą biedą i to spowoduje, że żadne wybory pewnie nie zostaną przeprowadzone w sposób właściwy.

To uważam za absurdalne i raczej w tym momencie nierealne. Chodzi o to, jak ma wyglądać przeprowadzenie wyborów w komisjach wyborczych, które są projektowane, jeśli w jednej komisji w przypadku gminy do 50 tys. mieszkańców może być od trzech do dziewięciu komisarzy. Ci ludzie będą to liczyć przynajmniej kilka dni.

Ja sobie tego nie wyobrażam. Poczta Polska może sobie z tym nie poradzić.

Dziękuję.

Proszę bardzo. Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Natomiast odnośnie do całej opozycji, która zabiera głos w sposób nieprawdopodobnie demagogiczny, chcę powiedzieć, że ja, szczerze mówiąc, już wolę słuchać PiS-u, niż słuchać tej potwornej demagogii, która leje się tutaj z ust przedstawicieli Lewicy i Koalicji Obywatelskiej.

Moim zdaniem ten gowinizm stosowany przejdzie do historii polskiego parlamentaryzmu. Ale, proszę państwa, Gowinowie przychodzą i odchodzą, a my zostaniemy z tymi wyborami, które będą, powiedzmy sobie jasno, komedią. Nie wierzymy PiS-owi, że uczciwie zrobi te wybory, dlatego będziemy głosowali przeciw.

Wysoka Izbo! Jeżeli was nie przekonują te głosy, które padały z tej mównicy, to na pewno taką czerwoną lampkę powinny zapalić u was słowa Janusza Korwin-Mikkego. Jak on zaczyna was popierać i doceniać, to się zastanówcie, czy dobrze robicie. To po pierwsze. Po drugie, kwestia bezpieczeństwa i rzetelności wyborów. O bezpieczeństwie mówiłem w pierwszym wystąpieniu. Teraz o rzetelności tych wyborów i staranności ich przeprowadzenia.

Mam pytanie do pani marszałek, czy skonsultowała te zmiany z Radą Dialogu Społecznego, z organizacjami związkowców i pracodawców, czy zasięgnęła opinii Państwowej Komisji Wyborczej na temat możliwości zrealizowania tego prawa przez Państwową Komisję Wyborczą. Czy zapytaliście związkowców, choćby Poczty Polskiej, jaka jest ich opinia na ten temat? To są podstawowe zasady prowadzenia dialogu społecznego w Polsce. Nie mówię już o dialogu obywatelskim, bo nie było żadnego wysłuchania publicznego, żadnej debaty, która powinna być, szczególnie przy tak ważnych projektach. A teraz o możliwościach technologicznych i technicznych przeprowadzenia tych wyborów.

To znaczy, że 26 tys. listonoszy ma dostarczyć. To są 583 adresy. Jeszcze raz zwracam uwagę na zgłaszanie się osób spoza terytorium Rzeczypospolitej, obywateli Rzeczypospolitej, którzy mają takie samo prawo do udziału w tych wyborach. Kwestia obwodowych komisji wyborczych.

Teraz ma to zastąpić jedna komisja. Wtedy składało się to z 4,5 tys. osób, teraz te głosy ma liczyć 45 osób. 4,5 tys. osób do tej pory liczyło głosy, a teraz ma je liczyć 45 osób w gminie miejskiej Kraków. To pokazuje, że nie ma szans na rzetelność przy przeprowadzeniu tego procesu. On jest po prostu nieprzygotowany. Kiedyś byliście przeciwnikami korespondencyjnego głosowania, dzisiaj powołujecie się na Bawarię. Tylko że w Niemczech wybory korespondencyjne przeprowadzane są od lat i poczta niemiecka wysyła zapytanie oraz materiały wyborcze przed każdymi wyborami. Ten system jest przygotowany i sprawdzony. Nie był przeprowadzany przecież w całym landzie, objął tylko część tego landu - w części landu była druga tura wyborów. W niektórych to się zakończyło na pierwszej.

Dziękuję, panie pośle.

Pani Marszałek! Panie Premierze! Wysoka Izbo!

Wtedy też były pewne siły - tak patrzę na zgromadzonych na sali, pewnie pan prezes najlepiej mógłby nam o tym opowiedzieć - które wychodziły na tę mównicę, tak samo wszczynały taką awanturę, w każdej sprawie obrażając każdego, kto tylko ma inne zdanie, i mówiły, że w zasadzie tego nie można zrobić, ale tutaj jest bezrobocie, czemu się tym nie zajmujecie. A w istocie to wszystko miało tylko jeden istotny cel - zablokować wszelkie zmiany. W istocie miało to tylko na celu restaurowanie postkomunizmu czy też instalowanie postkomunizmu w Polsce.

Konstatuję to z wielką przykrością, bo starałem się, tak samo zresztą jak poseł wnioskodawca, ani nikogo nie obrażać, ani nikogo nie atakować, tylko zachęcić państwa do merytorycznej dyskusji. Ale nieprawdą jest to, co państwo twierdzicie, i to, co tutaj mówiliście, powtarzając te same kłamstwa o tym, że wyborami żyje tylko nasz obóz. Powiem tak: przecież działania, które są podejmowane, są widoczne. Myślę, że jeszcze w tym tygodniu trafi do Wysokiej Izby kolejny projekt ustawy, który ma właśnie pomagać przedsiębiorcom, który ma pomagać służbie zdrowia, który ma pomagać różnego rodzaju grupom osób, które są dziś poszkodowane. Konstytucja nie przestała obowiązywać, życie nie przestało się toczyć. Sprawa druga. Cały czas pomimo tylu głosów nie usłyszeliśmy, co w istocie ma dać comiesięczna awantura o przesuwanie terminu wyborów, oprócz tego, że państwo będziecie mieli przez ten miesiąc wolne i nie będziecie w żaden sposób uczestniczyli w pracach i w żaden sposób nie będziecie podejmowali decyzji. Będzie to wyraźne złamanie, a co najmniej mocne nagięcie konstytucji i wreszcie uderzenie w gospodarkę, o którą rzekomo tak się troszczycie. Sprawa trzecia - konstytucja, 6 miesięcy przed. Przytoczę artykuł. Przytoczę nie artykuł, ale słowa z posiedzenia komisji sejmowej pana przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej, na którego się często powołujecie, pana Wojciecha Hermelińskiego, który sam w Sejmie, przedstawiając zmiany i zachęcając do nich, chociaż było mniej niż 6 miesięcy przed wyborami, twierdził: Jednak jestem skłonny stwierdzić, że trudno jest mówić o takich istotnych zmianach w prawie wyborczym, o których mówi orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Są to przede wszystkim kwestie techniczne, na których nam zależy. I z tego względu, co muszę powiedzieć, wyrażamy uznanie dla Wysokiej Izby i dla projektodawców, że te przepisy wprowadzają - itd. Tak że te słowa można by dzisiaj powtórzyć. Nie, zupełnie pan myli wszystko.

Otóż tak: gdyby wówczas, w grudniu 2017 r., ktokolwiek zapytał mnie, czy jestem za tym, żeby zakazać czy drastycznie ograniczyć możliwość wyjścia Polaków z domu, powiedziałbym, że oczywiście jestem przeciwko takiemu pomysłowi. Tak samo jak wówczas byłem - i dalej pozostaję - przeciwko wpisywaniu na stałe maksymalnego rozszerzania tego prawa. To jest ustawa, która się odnosi do tych wyborów. Jesteśmy w nadzwyczajnej sytuacji, a więc nadzwyczajne środki są wskazane. Dziwię się, że ktoś może tego nie rozumieć. Powiem tak, wychodząc naprzeciw: jeżeli to budzi wątpliwości, choć moim zdaniem jest jasne, że intencja jest zupełnie inna, nie żeby karać kogoś za to, że nie poszedł na wybory, ale jeżeli budzi to wątpliwości, składamy poprawkę, jedną z paru, która to ureguluje. Odnośnie do głosu pana przewodniczącego, że w Krakowie będzie problem z policzeniem głosów, panu przewodniczącemu umknął art. 10 ust. 11 projektowanej ustawy, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach komisarz wyborczy, mając na względzie sprawność i skuteczność pracy komisji (Dzwonek), może powołać w skład gminnej obwodowej komisji większą liczbę osób niż określona w ust. 5. Wysoka Izbo! Kończąc, zachęcam wszystkich mimo wszystko do poparcia tej ustawy w imię troski o Polaków, a jutro z tą samą werwą, determinacją byście państwo dyskutowali na temat pomocy Polakom, pomocy polskim firmom, polskim przedsiębiorcom i byście państwo nie uchylali się od pracy w Sejmie. Pan poseł Michał Szczerba.

Szanowna Pani Marszałek! Chciałbym złożyć wniosek formalny, art. 184 regulaminu Sejmu: zmiana w sposobie prowadzenia dyskusji. Szanowna Pani Marszałek! Ale w zasobie Biura Analiz Sejmowych jest opinia z 20 maja 2010 r., która mówi, w jakich okolicznościach pani może dokonać zmiany w swoim postanowieniu dotyczącym zarządzenia wyborów i wskazania daty wyborów. Te okoliczności to jest stan nadzwyczajny, to jest np. stan klęski żywiołowej. Nowelizacja postanowienia marszałka Sejmu jest to de facto nowe zarządzenie wyborów. Chciałbym, żebyśmy wszyscy wiedzieli, co się dzieje w tej chwili w domach pomocy społecznej. W domach pomocy społecznej w Drzewicy w Łódzkiem - 64 osoby zakażone, w Tomczycach - 70, Jakubowice - 40, Niedabyl - 16, Koszęcin - 17 (Dzwonek), Wola, przepraszam, Warszawa przy Bobrowieckiej zakład opiekuńczo-leczniczy - 19 osób, 16 DPS-ów w kwarantannie. Naprawdę państwo uważacie, że w takich okolicznościach można przeprowadzać wybory i umożliwić tym ludziom.

Jesteśmy już po dyskusji, panie pośle, i w tej chwili jesteśmy tylko przed pytaniami. Zamykam dyskusję. Pan poseł Robert Kropiwnicki, Koalicja Obywatelska. Proszę bardzo.

Otóż podstawą każdej demokracji są wolne wybory. A wy chcecie urządzić wybory z pistoletem przy głowie. Szantażujecie Polaków, że jak nie pójdą w czasie epidemii, w czasie zagrożenia życia na wybory, to się wasz świat zawali. Wasz - tak, wasz PiS-owski świat się może zawalić. Ale ludzie chcą przede wszystkim spokoju, chcą pracy i demokracja musi być świętem, a nie żałosną stypą, którą chcecie urządzić na grobach wielu ludzi. Naprawdę, ludzie się boją o swoje życie, ludzie tracą pracę, nie wiedzą, czy będą mieli wypłatę w maju, a wy mówicie: idźcie na wybory, bo my chcemy kasę. To jest skandal. Naprawdę jak dyktatura się zachowujecie i będziecie za to odpowiadać. Wszyscy dyktatorzy liczą, że są bezkarni. Każdy dyktator uważa, że jego to nie dotyczy. Proszę bardzo. Ja mam bardzo dużo pytań, więc do rzeczy. Czy w istocie przyzwolenie pani marszałek, żeby w trakcie trwania kampanii wyborczej zmieniała datę wyborów, nazywa pan drobną kwestią techniczną, a nie istotną zmianą w zasadach przeprowadzania wyborów? Po drugie, w jakim, przepraszam, trybie zamierzają państwo zmienić art. 17, skoro właśnie procedujemy nad tą ustawą? I co to jest za deklaracja, że to się nie znajdzie, jeżeli... po tej dyskusji i po wnioskach posła Krzysztofa Śmiszka? Napisaliście ustawę na kolanie, a teraz bez żadnego trybu będziecie ją korygować? Dlaczego w tej ustawie znajduje się kuriozalny zapis o tym, że to minister do spraw aktywów państwowych stanie się de facto Państwową Komisją Wyborczą? Dlaczego to PiS-owski minister Sasin ma decydować o kształcie i formie karty wyborczej, ale także o tym, co oprócz tej karty znajdzie się w pakiecie do głosowania, czy znajdzie się tam ulotka Andrzeja Dudy? Dlaczego chcecie zmuszać Polaków do głosowania pod karą więzienia? Bo nie wierzę w państwa deklaracje, że znajdziecie sposób (Dzwonek) na wycofanie tej poprawki. Dlaczego nie widzicie ryzyka, że przemocowy mąż będzie mógł zagłosować za żonę, babka za dziadka, ciotka za wujka? Pan poseł Marcin Kierwiński, Koalicja Obywatelska.

Wysoka Izbo! Do tej pory wybory w Polsce przeprowadzała Państwowa Komisja Wyborcza. To był gwarant niezależności i wolności tych wyborów. Jaki system proponuje PiS? Marszałek Witek z PiS ustali termin, który pasuje PiS-owi, według zapisów niezgodnych z konstytucją. Wicepremier z PiS przygotuje pakiety wyborcze. Co będzie w tych pakietach, to tylko minister Sasin wie. Były wiceminister z PiS, najbliższy współpracownik pana Błaszczaka, odbierze pakiety wyborcze od Polaków. No, może od niektórych Polaków, bo czy od wszystkich, to mamy poważne wątpliwości. A na koniec komisja powołana przez PiS policzy te głosy. Wszystko jest jasne. Partia organizuje wybory, partia organizuje wyniki tych wyborów. To nic innego jak system fałszowania wyborów. Dziękuję, panie pośle. Proszę bardzo, pani poseł Małgorzata Tracz, Koalicja Obywatelska.

Wysoka Izbo! Jest mi wstyd, że dziś jako Sejm debatujemy nad projektem zmian w ordynacji wyborczej. Jest mi wstyd przed Polkami i Polakami, którzy codziennie mierzą się z kolejnymi wyzwaniami, którzy tracą teraz pracę lub muszą likwidować swój biznes, którzy tracą środki do życia. Jest mi wstyd przed pracownikami służby zdrowia, którzy z narażeniem życia walczą na pierwszej linii z epidemią. Jest mi wstyd, że nie zajmujemy się rozwiązywaniem problemów Polek i Polaków, które dotykają ich tu i teraz. Zamiast tego zajmujemy się egoistycznymi interesami jednej partii i jednego kandydata - partii i kandydata, którzy, jak widać, za nic mają ludzkie zdrowie i życie, za nic mają zdrowie i życie wyborców i wyborczyń, pracowników poczty, pracowników komisji wyborczych. Przecie do tych wyborów, nie patrząc na bezpieczeństwo Polek i Polaków, nie patrząc na wolę Sejmu wyrażoną w głosowaniu o godz. 13. Dlatego też (Dzwonek) chciałam zapytać: W jaki sposób macie zamiar zabezpieczyć pracowników poczty, pracowników komisji wyborczych, wyborców i wyborczynie przed zakażeniem koronawirusem oraz zapobiec jego przenoszeniu dalej?

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Twórcy tej ustawy, wyjaśnijcie mi, czy już obstalowaliście te skrzynki specjalne, o które pan minister ma zadbać i sformułować wymagania, jakim powinna odpowiadać nadawcza skrzynka?

A poważna kwestia jest taka: Na jaki adres, jak rozumiem - już od jutra, wysyłacie te pakiety wyborcze do naszych rodaków, Polaków za granicą? Prawda, nie znacie tych adresów, a poczta nie doniesie.

Proszę bardzo, pan poseł Piotr Zgorzelski, PSL-Kukiz15. Proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Utrwalone orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego - i to w trzech swoich orzeczeniach - jednoznacznie stwierdza, że istotnych zmian z punktu widzenia prawa wyborczego nie wolno przeprowadzać na 6 miesięcy przed wyznaczeniem terminu wyborów. Mam taki test dla posłów Prawa i Sprawiedliwości. Złóżcie w tej kwestii zapytanie do tzw. Trybunału Konstytucyjnego. Bo jeszcze chyba tylko wy wierzycie lub udajecie, że wierzycie w to, że ta instytucja nosi przymioty konstytucyjne. Zabawna będzie ekwilibrystyka, z jaką ci sędziowie będą starali się udowodnić, że nie są to istotne zmiany, wszak dotyczą tylko 30 mln ludzi.

uważaliście w 2016 r. Zamykam dyskusję. Proszę państwa. Przepraszam. W związku z tym, że w czasie drugiego czytania zgłoszono. W związku z tym, że w czasie drugiego czytania zgłoszono do przedłożonego projektu ustawy poprawki, proponuję, aby Sejm przystąpił do trzeciego czytania projektu ustawy po doręczeniu paniom i panom posłom zestawienia poprawek. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Proszę państwa, wpłynął wniosek Koalicji Obywatelskiej o reasumpcję głosowania nr 39. Zgodnie z uchwałą nr 42 Prezydium Sejmu organem uprawnionym do oceny przesłanki, czy wynik głosowania na posiedzeniu plenarnym Sejmu budzi uzasadnione wątpliwości, co skutkować może reasumpcją głosowania, jest marszałek Sejmu. Oceny powyższej marszałek Sejmu dokonuje po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów. Dlatego ogłaszam teraz 5 minut przerwy i zapraszam. Wpłynął wniosek o reasumpcję głosowania, mam go przed sobą. Proszę bardzo.

Zgłaszaliśmy to wielokrotnie. Państwo dzisiaj chyba widzieliście, jakie niebezpieczeństwa niesie ten system. Powinna przeprowadzić ponowne głosowanie, ponieważ zachodzi uzasadniona obawa, że wyniki tego głosowania odbiegają od woli Wysokiej Izby. Głosują w systemie zdalnym, niestety system inaczej zagłosował.

W tym czasie zostaną państwu posłom doręczone poprawki.

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. Sejm przeprowadził pierwsze czytanie oraz podjął decyzję o niezwłocznym przestąpieniu do drugiego czytania projektu ustawy. Zestawienie zgłoszonych w trakcie drugiego czytania poprawek zostało paniom i panom posłom doręczone. Przed przystąpieniem do trzeciego czytania, proszę państwa, wyjaśnienie dotyczące wniosku, który wpłynął ze strony Koalicji Obywatelskiej, o reasumpcję głosowania nr 39. Przypomnę, że głosowanie nr 39 dotyczyło odrzucenia projektu w pierwszym czytaniu.

W związku z tym, proszę państwa, zgodnie z uchwałą, którą państwu przeczytałam wcześniej, po zwołaniu Konwentu Seniorów, zasięgnięciu opinii, tego wniosku nie przyjmuję. Przystępujemy, proszę państwa, do trzeciego czytania. W pierwszej kolejności poddam zgłoszony w dyskusji wniosek o odrzucenie projektu ustawy w całości.

Poddaję zatem pod głosowanie zgłoszony w dyskusji wniosek o odrzucenie projektu ustawy w całości. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem projektu ustawy zawartego w druku nr 328, zechce nacisnąć przycisk.

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił. Nad tym poprawkami głosować będziemy łącznie. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawek od 1. do 3., zechce nacisnąć przycisk.

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Stwierdzam, że Sejm poprawki przyjął. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki 4., zechce nacisnąć przycisk.

Stwierdzam, że Sejm poprawkę odrzucił. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 328, wraz z przyjętymi poprawkami, zechce nacisnąć przycisk.

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Sejm uchwalił ustawę o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. Hańba!